Wysoki Sejmie! Przychodzi nam głosować nad poprawkami senackimi do tarczy antykryzysowej. Chciałbym poprosić - ponieważ dostaliśmy informację, że głosowania będą zblokowane w zaledwie sześć głosowań, a tymczasem poprawek senackich jest znacznie więcej - o to, żeby nam wyjaśnić, nim przejdziemy do głosowań, jaki jest klucz merytoryczny zblokowania tych poprawek. Nasi analitycy, nasi eksperci starali się wypracować merytoryczną ocenę każdej z tych poprawek. Te regulacje, które rząd zaproponował, są niewystarczające, ale chcemy, żeby jak najszybciej zaczęły obowiązywać, dlatego prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób one zostały pogrupowane, żebyśmy mogli głosować zgodnie z kluczem merytorycznym, a nie na opak czy w jakiś sposób nie do końca możliwy do przewidzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo proszę.

Dziękuję. Ja tylko wyjaśnię panu posłowi, że zblokowanie nastąpiło na podstawie uchwały nr 4 Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie wykładni art. 50 ust. 6 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Finansów Publicznych przedłożyła sprawozdanie o uchwałach Senatu. Nie zauważyłam. Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

Udało się wprowadzić kilka ważnych, merytorycznych poprawek dotyczących wyższej płacy i konieczności płacenia przez państwo 75% wynagrodzenia pracodawcom, spraw związanych z odroczeniem ZUS-u i płatności za rachunki, spraw dotyczących podwyższenia wynagrodzenia o 50% dla personelu medycznego. Nie możemy tego odrzucić w jednej poprawce. Prawa pracownicze i prawa przedsiębiorców powinny dzisiaj w tej Izbie wybrzmieć. Jeżeli chcemy dzisiaj debatować o tarczy antykryzysowej, a nie tarczy tekturowej, to niezbędna jest debata, a nie szybkie głosowanie i do domu. Dziękuję bardzo. Proszę. Pani Marszałek!

Zgłaszam wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad. To, co dzieje się w tej chwili w Wysokiej Izbie, jest niedopuszczalne. Senat postanowił załatać dziurawą rządową tarczę, wprowadzając rzeczywistą tamę, która ma przeciwdziałać kryzysowi.

Polacy nie dowiedzą się, kto z was głosował w haniebny sposób, odrzucając dobre rozwiązania dla polskich pracowników. Jednocześnie w sposób skandaliczny, wbrew jakimkolwiek zwyczajom parlamentarnym ucina się dyskusję. Chodziło o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji poprzez umożliwienie zadawania pytań. To jest moja kompetencja. To jest dyspozycja marszałka Sejmu.

Dziękuję bardzo. W imieniu Koalicji Polskiej chciałbym powiedzieć, że nie możemy zgodzić się na taki sposób prowadzenia obrad: bez pytań, bez dyskusji, bez możliwości przedstawienia jedynej szansy na to, żeby ustawa antykryzysowa zadziałała, żeby pomogła pracownikom, pracodawcom, rolnikom, przedsiębiorcom, wszystkim, którzy dzisiaj czekają na decyzję Izby, czekają na mądrą decyzję. Zerwaliście z zasadą solidarności. Nie chcecie współpracy, interesuje was tylko i wyłącznie ustawka pod wybory i likwidacja Rady Dialogu Społecznego, likwidacja dialogu społecznego w Polsce.

Nie wprowadzacie tych zmian, zblokowaliście je i chcecie je odrzucić.

Komisja Finansów Publicznych przedłożyła sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie: - ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 311, - ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, druk nr 310, - ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju, druk nr 312. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych uchwał. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. W związku ze zgłoszonym sprzeciwem do art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu sprawę tę rozstrzygniemy w głosowaniu. Kto z pań i panów posłów jest za skróceniem terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu, zechce nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął. Wysoka Izbo! Zgłoszono wniosek o przeprowadzenie łącznej dyskusji nad uchwałami Senatu zawartymi w drukach nr 310, 311 i 312 w wymiarze 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 307 i 311) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Panie Premierze! Wysoka Izbo! Senat do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na posiedzeniu zakończonym w dniu dzisiejszym wniósł 81 poprawek. Pani marszałek skierowała w dniu dzisiejszym uchwałę Senatu do Komisji Finansów Publicznych. Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyła uchwałę Senatu. W czasie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych dyskusja była obszerna, wszyscy posłowie mogli się wypowiadać na temat uchwały Senatu. Dyskusja trwała ok. 5 godzin.

Poprawki dotyczyły kilku grup, m.in. znaczących wydatków finansowych w różnych dziedzinach - przywoływanych tu już 20 mld, ale jeszcze wielu, wielu innych. Brak precyzyjnych określeń źródeł finansowania tych wydatków i świadomość tego, że rząd jest odpowiedzialny za budżet, a równocześnie deklaracja, że jeszcze nie jest to zakończenie procesu legislacyjnego i pomocy rządowej dla poszkodowanych z tytułu epidemii koronawirusa, poszkodowanych gospodarczo - stąd komisja przyjęła zasadę, że jeśli nie jest w stanie oszacować wydatków, to zostawia tę decyzję i rekomendację rządowi, tak aby w sposób odpowiedzialny można było te wszystkie wydatki i tę pomoc deklarować. Natomiast wszystkie wnioski Senatu - aczkolwiek w swoim założeniu słuszne - niemające pewnych źródeł finansowania nie mogły zostać zaakceptowane. Pragnę zaznaczyć, że ta dyskusja nie dotyczyła meritum sprawy, nikt nie mówił, że np. złym rozwiązaniem jest umożliwienie głosowania korespondencyjnego tym, którzy są poddani kwarantannie, w kontekście braku wiedzy, kiedy naprawdę będą wybory, w jakich okolicznościach będą wybory i jak długo będzie trwała epidemia. Stąd ten zapis na pewno będzie zapisem bardzo korzystnym i przydatnym dla tych, którzy będą poddani obowiązkowej kwarantannie.

Pozostałe poprawki komisja proponuje odrzucić. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. Proszę bardzo, wniosek formalny. Wysoka Izbo! Składam w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej wniosek formalny o odrębne, rozdzielne głosowanie nad każdą poprawką Senatu. To zbyt ważne, byście państwo do porządku dziennego przechodzili nad tym, by w jednym głosowaniu odrzucić 20 mld zł na służbę zdrowia, odrzucić równe traktowanie polskich pracowników i zagwarantowanie wszystkim świadczeń na wypadek kryzysu. To absolutnie niewybaczalne, że chcecie bez dyskusji pozbawić opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia świadczeń w czasie, gdy muszą sprawować opiekę. To również absolutnie niedopuszczalne, byście chowali się za tabletami, gdy chcecie odrzucić realną pomoc w postaci 40 tys. zł, a nie zaproponowanych 5 tys. zł, dla polskich przedsiębiorców. To absolutnie niedopuszczalne, by z tej mównicy nie zabrać głosu i nie powiedzieć, dlaczego nie chcecie dodatkowych środków z Unii Europejskiej m.in. na doposażenie polskich szpitali. I wreszcie, szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo (Dzwonek), to jest to miejsce, w którym pan premier Morawiecki powinien wstać i powiedzieć Polakom: Oszukaliśmy was.

zastosowanie uchwały nr 4 Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie wykładni art. 54 ust. 6 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Odrzucenie tej propozycji będzie oznaczać, że Sejm przyjął wniosek o oddzielne głosowanie nad każdą poprawką. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji łącznego głosowania nad poprawkami, proszę nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm przyjął propozycję łącznego głosowania nad poprawkami zgodnie z wcześniej przedstawioną propozycją.

Komisja wnosi o odrzucenie tych poprawek. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

Komisja wnosi o przyjęcie tych poprawek. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druki nr 306 i 310) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Senat w swojej uchwale proponuje 10 poprawek do tej ustawy. Pani marszałek skierowała uchwałę Senatu do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych.

Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Proponuję zastosowanie uchwały nr 4 Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca. Dzień dobry, pani marszałek, po raz kolejny. Wysoka Izbo! Kolejny raz w imieniu Koalicji Obywatelskiej proszę o to, żebyście państwo dopuścili w tej Izbie do dyskusji. Przed chwilą głosami posłów koalicji rządzącej, większości odrzuciliście państwo bardzo istotne poprawki, które Senat wniósł do tej ustawy. Zagwarantowaliśmy realną pomoc polskim pracodawcom. Tymczasem państwo pod osłoną własnych tabletów dopuszczacie do tego, że na dniach będą zwalniani pracownicy, ludzie będą tracić pracę, podczas gdy wy w ciszy zabijacie nie tylko nadzieję, ale też przede wszystkim elementy polskiego parlamentaryzmu. Na to nie może być zgody. Nie może być zgody na oszustwo, na wielkie oszustwo nie tylko w sprawie tarczy, ale też przede wszystkim w sposobie obradowania.

Panie pośle, to nie jest wniosek, który poddam pod głosowanie, ponieważ to jest wniosek o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji, a nad tym wnioskiem już głosowaliśmy. Proponuję zastosowanie uchwały nr 4 Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie wykładni art. 54 ust. 6 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem przedstawionej przeze mnie propozycji łącznego głosowania nad poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję przyjął. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o ich przyjęcie.

Nikt nie był za, 454 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druki nr 308 i 312) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo!

Komisja po przeanalizowaniu poprawki rekomenduje poprawkę przyjąć. Dziękuję bardzo.

Dziękuję, pani marszałek. Wysoka Izbo! To ostatnie głosowanie. Demokracja umiera w ciszy. Ta cisza jest symbolem tego rządu. Wnoszę o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów celem zmiany porządku obrad i włączenie do porządku obrad informacji rządu na temat obecnej sytuacji związanej z walką z koronawirusem. Tak jak powiedziałem, tu powinien stać premier. Dlaczego przyjęliście błędną metodologię, jeżeli chodzi o statystyki? Dlaczego boicie się odpowiedzi na najważniejsze pytania? Dlaczego lekarze, pielęgniarki, służba zdrowia nie mają podstawowych środków ochrony? Dlaczego oszukujecie miliony pracowników, twierdząc, że będzie dla nich jakakolwiek pomoc? I wreszcie dlaczego wbrew obietnicom dialogu i współpracy odrzuciliście państwo wszystkie dobre poprawki Senatu? Dziękuję, panie pośle.

Panie Premierze! Gdyby była dyskusja, nie byłoby wniosków formalnych. Taka jest prawda.

Dzisiaj miliony Polek i Polaków oczekują wsparcia, dobrego słowa, myślenia o tym, jak chcemy im pomóc, wytłumaczenia, dlaczego coś się nie uda, bo nie wszystko się uda. Nie róbmy z Sejmu zabawki, która ma służyć 235 parlamentarzystom, którzy powiedzieli reszcie: Nie będziecie debatowali.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Nikt nie był za, 455 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.